posiedzenie. Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Martę Kubiak, Krzysztofa Kubowa, Piotra Olszówkę i Rafała Webera. W pierwszej części obrad sekretarzami będą posłowie Piotr Olszówka i Krzysztof Kubów. Protokół i listę mówców prowadzić będą posłowie Krzysztof Kubów i Marta Kubiak. Protokół 74. posiedzenia Sejmu uważam za przyjęty wobec niewniesienia zastrzeżeń. Proszę o chwilę uwagi.

Stwierdzam, że pan poseł Piotr Józef Müller złożył ślubowanie poselskie. Rada Ministrów przedłożyła autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Autopoprawka ta została paniom i panom posłom doręczona w druku nr 3112-A. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę rozumiał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół w dyskusji w pierwszym czytaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Informuję, że w związku z niezgłoszeniem przez uprawnione podmioty tematu informacji bieżącej oraz pytań w sprawach bieżących punkty te nie zostaną rozpatrzone na bieżącym posiedzeniu Sejmu. Punkty porządku dziennego bieżącego posiedzenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów. Informacja w tej sprawie, a także wykaz ustaw, które Senat przyjął bez poprawek, dostępne są w Systemie Informacyjnym Sejmu.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Spotykamy się dzisiaj tutaj, żeby rozstrzygnąć o jednej bardzo ważnej sprawie, o sprawie związanej. z cenami energii, z czymś, co interesuje Polaków. I tutaj bardzo interesują Polaków również okoliczności, które doprowadziły do tego stanu, w jakim dzisiaj jesteśmy.

Jak mogliście doprowadzić do takiego stanu, do takich podwyżek między rokiem 2008 a rokiem 2012? Bardzo łatwo można sobie to sprawdzić. Tymczasem, szanowni państwo, [[Dzwonek]] dzisiejsza sytuacja nie wzięła się z niczego. i jest skutkiem szalejących cen hurtowych energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Po drugie, oczywiście braku odpowiedniego wynegocjowania pakietu klimatycznego przez rząd Platformy Obywatelskiej. Nasz rząd jeszcze w poprzednim okresie, w roku 2017, zajął się tym tematem, pracował nad miksem energetycznym. Zaproponowaliśmy pewną strategię, która w najbliższych kilku latach, drodzy rodacy, doprowadzi do tego, że będziemy mieli.

Ale to nas nie zadowala. Chcemy, żeby one były na poziomie stabilnym względem pierwszej połowy 2018 r.

Otóż wasza pani wiceminister z Ministerstwa Środowiska stwierdziła, że policzyliście te skutki dla gospodarki polskiej po przyjęciu pakietu w 2008 r., a nie przed.

Otóż liczył to Bank Światowy, szanowni państwo. Bardzo szacowna instytucja, my oczywiście bardzo szanujemy Bank Światowy, ale żeby rządu ówczesnego, waszego. nie stać było na to, żeby policzyć z własnych źródeł, wypracować własne analizy, opracowania. My, szanowni państwo, wprowadzamy rozwiązania, które tutaj będą dyskutowane. Bardzo konkretne. Rozwiązania, które mają doprowadzić do utrzymania cen energii na poziomie pierwszej połowy 2018 r.

Będzie jeszcze mniej w rachunkach za energię elektryczną w postaci naliczonego podatku VAT. Czyli VAT, akcyza i opłata przejściowa to jest jeden pakiet czy jedna część naszego rozwiązania. Jeszcze dodatkowo, chcemy to bardzo wyraźnie podkreślić, dla samorządów, dla firm w tych przypadkach, gdzie firmy prywatne, dystrybucyjne firmy prywatne już wypracowały jakieś nowe kontrakty czy uzgodniły nowe kontrakty z samorządami, tworzymy mechanizm powrotu do cen sprzed 1 lipca 2018 r. Tak, ciekawe, jak zagłosuje ta druga część sali. Za naszą ustawą, która prowadzi do tego, że rzeczywiście dbamy o to, jakie są portfele Polaków. Dbamy o to, żeby ceny energii elektrycznej nie szły do góry, a w waszych czasach przez 4 lata poszły o 50% do góry. Dlatego wypracowujemy też metody, które są również ujęte w proponowanej ustawie, tak żeby można było zrekompensować.

I warto to podkreślić, szanowni państwo, że już dzisiaj mamy w Unii Europejskiej jedne z najniższych cen dla gospodarstw domowych, ale utrzymujemy je na tym poziomie. Nie doprowadzimy do wzrostu cen energii. Te rozwiązania będą też dobre dla samorządów i chcę to z całą mocą podkreślić, bo są dzisiaj, szanowni państwo, samorządy, zwłaszcza niektóre samorządy rządzone przez Koalicję Obywatelską, przez Platformę Obywatelską, które chcą wykorzystać jako pretekst to, że się rozpoczęła dyskusja wokół cen energii - uwaga - i chcą, drodzy rodacy, podnosić cenę za wywóz śmieci. Te samorządy chcą podnosić cenę za wodę, a nawet za transport publiczny, jak słyszałem, np. w jednym z większych miast Polski. Nie dopuśćmy do tego. Pilnujmy tych włodarzy, żeby oni teraz również dbali o portfele Polaków, tak jak o portfele Polaków dba rząd Prawa i Sprawiedliwości. A więc czując odpowiedzialność, panie marszałku, Wysoka Izbo, za Rzeczpospolitą, naprawiamy błędy naszych poprzedników. Błędy, które się tak mocno objawiły w rosnącej cenie uprawnień do emisji CO2.

Gdybyście chociaż część tej energii, z jaką jeździcie czy wypracowujecie donosy i różnego rodzaju, prawda, odezwy do Brukseli. część tej energii spożytkowali na prace nad systemem energetycznym. sytuacja dzisiaj byłaby zupełnie inna. Dlatego właśnie nasz rząd bierze ten problem i rozwiązuje go.

Ale równie, przede wszystkim, dbamy o to, żeby nie wzrosła cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, o to, o co państwo nie zadbaliście w latach 2008–2012, podnosząc cenę dla gospodarstw domowych o 50%. Wysoka Izbo! Dziękuję bardzo panu ministrowi Tchórzewskiemu oraz wszystkim posłom Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, którzy wypracowali rozwiązania w tym trudnym czasie, kiedy rzeczywiście polityka klimatyczna, błędy naszych poprzedników doprowadziły do tego stanu, w jakim jesteśmy. Rozwiązania, które proponujemy Polakom, są dobre, mają w sobie dobrą energię, zawierają zobowiązanie do tego, żeby cena energii nie rosła. Prosimy tylko, żeby pilnować tych różnych włodarzy w samorządach, żeby nie wykorzystywali tego pretekstu, który znika, do podnoszenia cen różnych usług publicznych. My ze swojej strony zadbaliśmy o to, żeby portfele Polaków nie ucierpiały z powodu błędów polityki klimatycznej, energetycznej naszych poprzedników. Bardzo dziękuję naszym posłom, naszemu panu ministrowi za zaproponowanie bardzo dobrej oferty dla Polaków.

Dziękuję panu premierowi. Zgłosili się panowie posłowie z wnioskami formalnymi.

Muszę zobaczyć ten wniosek formalny, czy. Jeżeli nie ma na piśmie.

Wysoka Izbo! Składam wniosek formalny o przerwę do godz. 12, o zwołanie Konwentu Seniorów i rozszerzenie porządku obrad o ustawę, która wprowadzi 98-procentową bonifikatę na gruntach Skarbu Państwa. Pan poseł Kaczyński na partyjnym wiecu mówił, że brak tej 98-procentowej bonifikaty to jest rabowanie Polaków. Panie Prezesie Kaczyński! Dajemy panu szansę, panu i panu premierowi Morawieckiemu, [[Oklaski]] aby w tym zakresie rząd, na którego czele stoi Mateusz Morawiecki, akurat na tym małym odcinku nie rabował Polaków, żebyście nie byli grupą, która rabuje Polaków.

Panie marszałku... [[Poruszenie na sali]] ...w trybie wniosku formalnego. Ta ustawa jest naprawdę, szanowni państwo, bardzo, bardzo krótka. Dziękuję panu posłowi. Jest wniosek o przerwanie posiedzenia.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Proszę pana posła sekretarza o odczytanie komunikatu. Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenie Komisji Ustawodawczej - godz. 11.30. Dziękuję. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 3112 i 3112-A)

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoki Sejmie!

Dlatego też z tego miejsca chciałbym panu marszałkowi podziękować za zwołanie dodatkowego posiedzenia Sejmu w celu rozpatrzenia rządowego projektu ustawy, którego celem jest niedopuszczenie do wzrostu cen energii dla odbiorców energii elektrycznej w Polsce. O tym, jak ważna jest to kwestia nie tylko dla posłów koalicji rządzącej, ale także innych, świadczą projekty ustaw złożone przez inne kluby parlamentarne. Dlatego wyrażam przekonanie, że uda nam się dzisiaj wspólnie wypracować najbardziej korzystne rozwiązania dla polskich gospodarstw domowych, krajowych przedsiębiorstw, samorządów oraz pozostałych odbiorców. Ceny energii elektrycznej rosną w całej Europie. Wzrosty te silnie związane są z prowadzoną w Unii Europejskiej polityką klimatyczną. Głównym jej elementem jest system handlu przydziałami uprawnień do emisji gazów cieplarnianych ustanowiony na obszarze Unii Europejskiej dyrektywą z października 2003 r. Nakłada ona obowiązek zakupu uprawnień do emisji CO2 przez instalacje spalania paliw, wszystkie instalacje.

Są państwa, jak np. Niemcy czy Dania, gdzie ceny za tę energię były przynajmniej dwukrotnie wyższe. W projekcie ustawy zdecydowaliśmy się zaproponować program składający się z czterech interwencji, które pozwolą ustabilizować ceny energii elektrycznej w 2019 r. oraz dotrzymać danego słowa, że nasi obywatele nie muszą obawiać się wzrostu rachunków za energię elektryczną, bo takiego wzrostu dzięki ustawie, nad którą dzisiaj procedujemy, nie będzie. Projekt jest o tyle ważny, że będzie dotyczył wszystkich odbiorców w kraju, a zatem ok. 17,5 mln odbiorców energii elektrycznej: gospodarstwa domowe, samorządy, przedsiębiorstwa, szpitale, hospicja czy domy dziecka - wszystkich odbiorców. Mamy więc do czynienia z projektem ustawy o najwyższym znaczeniu społecznym i gospodarczym. Teraz chciałbym omówić te zaproponowane cztery interwencje mające na celu utrzymanie ceny energii elektrycznej w 2019 r. na poziomie z roku 2018.

Drugim działaniem jest obniżenie opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej o 95%. Dzięki tej zmianie rachunki za energię elektryczną odbiorców w Polsce zmniejszą się o 2240 mln zł. Trzecią zmianą, którą wprowadza ustawa, jest bezpośredni zwrot utraconego przychodu spółkom obrotu. Na ten cel zaplanowano ok. 4 mld zł, które zostaną wypłacone - na wniosek spółek obrotu, na wniosek tych, którzy uznają, że ponieśli szkodę - przez specjalnie powołany do tego Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Dzięki temu mechanizmowi przy przedstawieniu rachunku za energię elektryczną dla odbiorców... pozostawimy właściwie cenę rachunków za energię elektryczną dla odbiorców na poziomie z roku 2018 i nie ucierpi na tym interes spółek energetycznych - zarówno tych spółek, na których wpływ ma państwo, jak i tych wszystkich prywatnych spółek, które zajmują się obrotem energią elektryczną. Ostatnim, czwartym elementem zaproponowanego mechanizmu jest przeznaczenie ok. 1 mld zł na inwestycje prośrodowiskowe, dzięki którym zmniejszy się emisyjność naszej gospodarki. Środki te zostaną skierowane do krajowego systemu zielonych inwestycji. W zaproponowanym projekcie ustawy terminem odniesienia, w którym ceny energii elektrycznej dla odbiorców nie były jeszcze na ścieżce wzrostowej, jest 30 czerwca 2018 r. Dlatego w projekcie ustawy zaproponowano mechanizm zmiany dotychczas zawartych umów, tak aby nie zostali pokrzywdzeni odbiorcy energii elektrycznej, którzy w II półroczu zawarli niekorzystne dla nich kontrakty. Dotyczy to także samorządów, które najbardziej wskazywały na straty i problemy, które z tego tytułu je dotknęły.

Z tego tytułu spodziewamy się pozyskać ok. 5 mld zł.

Kolejnym źródłem finansowania będzie obniżenie wpływów do budżetu z tytułu obniżki podatku akcyzowego o 1850 mln zł.

Takie dodatkowe środki zostaną wykorzystane do tego, żeby nasi rodacy, gospodarstwa domowe, przedsiębiorcy, samorządy tyle mniej zapłacili za prąd w przyszłym roku.

Zatem przygotowane przez nas rozwiązanie jest kompleksowe. Polega ono na obniżce podatku, obniżce opłat stałych oraz zapewnia brak wzrostu cen energii przy zrównoważeniu interesów spółek energetycznych oraz odbiorców energii. Szanowni Państwo!

Dlatego też uważam, że to, co przygotowaliśmy, rozwiązuje bardzo ważny problem społeczny i gospodarczy w Polsce. Dziękuję panu ministrowi.

Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest ochrona polskich rodzin, polskich firm, przemysłu i samorządów przed negatywnymi skutkami skokowego wzrostu cen energii elektrycznej, jaki obserwujemy w całej Europie. Zaznaczmy, że w wielu krajach Europy mamy do czynienia ze wzrostem cen energii o kilkadziesiąt procent. W Polsce nie możemy się zgodzić na to dlatego, że uderzyłoby to i w indywidualnych odbiorców, i w gospodarkę, której rozwój jest naszym powodem do dumy. To właśnie ochrona portfeli i kieszeni Polaków, a także zapewnienie stabilnych dostaw energii w celu dalszego wzrostu gospodarki jest naszym obowiązkiem. Dzięki tej ustawie ceny prądu nie wzrosną. Utrzymamy je na dotychczasowym, akceptowalnym poziomie. Parasol ochronny, jakim jest proponowana przez rząd ustawa, jest na tyle szeroki, że zatrzyma ceny wszędzie tam, gdzie pojawia się presja podwyżki: od gospodarstw domowych po przedsiębiorstwa i samorządy. Rekordowy wzrost cen energii elektrycznej, przed którym musimy się chronić, jest wprost związany z polityką klimatyczną prowadzoną przez Unię Europejską.

Szczegółowo przedstawił to pan minister Krzysztof Tchórzewski.

Ta fala wzrostu cen uderzyła już dość mocno w Europejczyków. Zgodnie z zapowiedziami rząd wypracował i przedstawił konkretne rozwiązania, które - co ważne - dają gwarancję natychmiastowego działania. Szczegółowe założenia do projektu ustawy przedstawił pan minister Krzysztof Tchórzewski.

Wysoka Izbo! Nasze ceny prądu muszą być konkurencyjne. Polacy nie mogą płacić zbyt wysokich rachunków za energię elektryczną. Polskie firmy muszą mieć możliwość konkurowania na rynku Unii Europejskiej, a ceny prądu są tu kluczowe. Jednocześnie musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo energetyczne, czyli o rozwój naszego sektora energetycznego. Prawo i Sprawiedliwość twardo stoi na stanowisku, że koszt energii musi stanowić przewagę konkurencyjną naszej gospodarki. Dotrzymujemy słowa, jakie daliśmy Polakom, że w roku 2019 ceny prądu nie wzrosną. I wszystkich państwa niezależnie od tego, po której stronie sali państwo siedzicie, zapraszamy do przyłączenia się do tych korzystnych i potrzebnych działań. Zabezpieczenie Polaków przed drogą energią powinno być ambicją całej Wysokiej Izby. Nie warto robić polityki kosztem Polaków. Jest to też okazja dla naszych poprzedników do naprawienia błędu, jakim była zgoda na niekorzystne dla Polski rozwiązania w zakresie handlu uprawnieniami do emisji CO2. Szansa na to, żeby na Nowy Rok dać Polakom prezent, na który czekają: merytoryczną pracę, dobrą ustawę i zastrzyk dobrej energii na każdą kieszeń. To jest także okazja, żeby Wysoka Izba pokazała dziś milionom polskich odbiorców prądu, że stać ją na zgodną, merytoryczną pracę w tak ważnej sprawie. Prawo i Sprawiedliwość będzie głosowało za projektem ustawy przedstawionym przez rząd. W imieniu klubu Platforma Obywatelska pan poseł Sławomir Neumann. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wasza polityka energetyczna to polityka trzech „A”: amatorska, arogancka i anachroniczna. Wasz miks energetyczny to wysokie rachunki za prąd, które muszą płacić Polacy, polskie przedsiębiorstwa i samorządy. Co do odpowiedzialności poprzedników jeden cytat: Moja polityka dawała rezultaty, ale wielu się nie podobała. Musiała się nie podobać, bo my robiliśmy to, co w naszym interesie. Czy ja w Unii Europejskiej nie byłem solidarny? Przecież zgodziłem się na politykę klimatyczną z punktu widzenia Polski ryzykowną. To był mój gest w stosunku do pani kanclerz Angeli Merkel - 2007 r., prezydent Lech Kaczyński na posiedzeniu Rady Europejskiej. To w ramach odpowiedzialności za politykę klimatyczną poprzedników, panie premierze. Dzisiaj zapaliła wam się lampka, zwoje zaczęły pracować, zaiskrzyło i doszło do oświecenia, że pomysł na podwyżkę w wysokości kilkudziesięciu procent za prąd w roku wyborczym wam się nie opłaci. Potem może być drogo, to już was nie interesuje. To wasze kolejne oszustwo energetyczne. Wysokie ceny prądu to tylko i wyłącznie wasza wina i odpowiedzialność. To wina 3 lat waszej działalności w energetyce. Dzisiaj Polska ma na giełdach jedne z najwyższych cen energii w Europie, w Unii Europejskiej. Te rządy, wasze rządy zahamowały, a czasami wręcz likwidują politykę energetyki opartej na OZE, na odnawialnych źródłach energii.

Premier i minister energii mówią o tym, że do 2035 r. wszystkie wiatraki w Polsce będą zezłomowane. To jest wasza polityka względem OZE. Zmuszacie je do różnych haraczy na swoje polityczne imprezy, do dotowania waszych fundacji, do dotowania waszych stowarzyszeń, do topienia miliardów w nierentowne inwestycje. Gdy przejmowaliście rządy w 2015 r., wartość czterech spółek energetycznych była o kilkadziesiąt procent wyższa niż dzisiaj. Co to oznacza?

Oczywiście, że nie. To nie żart. Nie uchroniło ich to przed wyrzuceniem z pracy, ale przynajmniej próbowali. Jak myślicie, podziałało? Taki macie boski prąd. Minister Tchórzewski nie daje za wygraną i idzie dalej. W sierpniu tego roku zawierza Matce Boskiej wszystkie sprawy energetyki.

Polska nie potrzebuje cudu, żadnego boskiego cudu. Nie potrzebuje boskiego prądu, tylko taniego prądu. Żeby to zrobić, wystarczy was i waszych prezesów wyrzucić z roboty, tych nieudaczników i amatorów. Żadne cuda nie są potrzebne. Zmusiliście te firmy do wielomiliardowych nakładów na polski węgiel.

W tym roku już ponad 10 mln t rosyjskiego węgla wjechało do Polski. To jest wasza polityka energetyczna. Panie ministrze, szef Urzędu Regulacji Energetyki doniósł do prokuratury, że spółki, te największe spółki państwowe, [[Dzwonek]] prawdopodobnie podnosiły w ostatnim półroczu cenę energii na giełdzie w sposób niespotykany, tj. o kilkadziesiąt procent.

Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Rozpatrujemy dzisiaj projekt o próbie utrzymania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Zarysujmy obecny kontekst społeczno-gospodarczy. Czwarty rok kadencji dla każdej partii władzy jest bardzo trudny.

Cały czas mamy sytuację nieprawdopodobnej różnicy, jeżeli chodzi o zarobki. podnosi ZUS o ponad 100 zł dla drobnych przedsiębiorców. Zamrożona pozostaje kwota wolna od podatku PIT, najniższa w Europie, na poziomie 3091 zł. Do nowożeńców zostało rozesłanych kilkaset pism z pytaniem, ile dostali w kopertach. Nie myślicie o tym, jakie będą konsekwencje waszej polityki socjalnej plus imigracyjnej. Szerzy się nepotyzm i kumoterstwo na nieprawdopodobną skalę. To jest typowe dla każdej partii władzy w czwartym roku. W związku z tym obsadzacie swoimi znajomymi, rodzinami spółki Skarbu Państwa.

Wracając do tej ustawy, czyli ustawy o próbie utrzymania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, Kukiz’15 jako jedyna opozycja merytoryczna w Sejmie VIII kadencji przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i podatku VAT 2 tygodnie temu, tydzień przed rządem. Zaproponowaliśmy cięcia na podobnym poziomie opodatkowania energii elektrycznej, z tym że my zaproponowaliśmy obniżenie akcyzy do najniższego poziomu wymaganego przez Unię Europejską, czyli 1 euro. Pytanie, dlaczego w waszej ustawie jest 5 zł, a nie 1 euro.

Będziemy ten projekt ponawiać. Niestety mimo naszych próśb marszałek nie dopuścił do rozpatrywania projektu klubu Kukiz’15 równolegle z obecnym projektem. Jeżeli chodzi o ten projekt, który ma umniejszyć wpływy do budżetu o 9 mln zł - i dobrze, dlatego że nam zależy, żeby te pieniądze zostawały w kieszeniach obywateli, a nie były wydawane przez rząd - to może przytoczę komentarz, który pojawił się 2 godziny temu w Internecie: To są jaja nad jajami. Za 2 godziny Sejm ma zająć się ustawą prądową, ale już inną. Rząd przysłał autopoprawkę, która wywraca system ustalania cen, tworzy nowy fundusz wyrównania, zmienia już zawarte umowy itd. Bo zaraz głosujecie. Rękę w górę, kto czytał ten projekt. A więc właśnie. Szanowni Państwo! Autopoprawka, która pojawiła się wczoraj, liczy 12 stron. Tak, szanowni państwo, nie można tworzyć prawa. Jestem przekonany, że zbierzemy się znowu na początku roku i będziemy tę ustawę poprawiać, bo po prostu w ten sposób prawa się nie stanowi. Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, które po dniu 30 czerwca 2018 r. zawarło umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowe, jest obowiązane do zmiany warunków tej umowy nie później niż do dnia 1 kwietnia, ze skutkiem od dnia 1 stycznia. Szanowni Państwo!

Panie Marszałku! Szanowny Nieobecny Panie Premierze! Zabierając głos w imieniu Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów, chciałem zapytać, co się panu stało, panie premierze, że po tak koncyliacyjnym spotkaniu przedświątecznym Prawa i Sprawiedliwości i zaproszeniu opozycji do współpracy, po tak radosnych świętach Bożego Narodzenia wyszedł pan tu dzisiaj na trybunę sejmową i nie tylko obrażał pan swoich konkurentów politycznych, ale też kontynuował pan kampanię kłamstw realizowaną w czasie wyborów samorządowych. Panie Premierze! Pan tu przed chwilą z trybuny sejmowej mówił: przez ostatnie 8 lat ceny energii w Polsce wzrosły o 50%. Powtarzał pan to wielokrotnie.

ale inflacja w tym czasie wynosiła 18%. Czemu ma służyć to, co pan tu z tej trybuny sejmowej w taki sposób nam prezentował? Jeśli już coś rosło w ostatnich latach, to, panie premierze, na pewno wzrósł import gazu z Rosji.

Chcę zwrócić uwagę, że w roku 2015.

Czy panu nie wstyd, że finansuje pan imperialną politykę Putina? Mówicie o grzechu zaniedbania. Tak, mamy do czynienia z wielkim grzechem zaniedbania, bo pan premier i ministrowie odpowiedzialni za energetykę przez ostatnie co najmniej 6 miesięcy jeździli po kraju i zajmowali się kampanią wyborczą, zamiast rozwiązać problem, który sami stworzyli.

Wtedy pan Krzysztof się cieszył, że jest dewidenda.

Czy spółki oszukiwały pana? Czy pan oszukiwał premiera? Czy wszyscy razem chcieliście oszukać nas, społeczeństwo? Jeśli prezes Urzędu Regulacji Energetyki składa doniesienie do prokuratury na zmowę cenową proponowaną przez spółki nadzorowane przez pana premiera, to pytanie, czy minister Ziobro rzeczywiście to wyjaśni.

A więc zamiast przechodzenia na zieloną stronę mocy, zamiast budowania energii odnawialnej, wy tę energię odnawialną wycofywaliście. Mówicie o projekcie budowy elektrowni jądrowej. W to miejsce można zbudować 3 tys. biogazowni o mocy 1 M i oddać do użytku w ciągu 3 lat maksymalnie za cenę co najmniej o 20% niższą. Na poprzednim posiedzeniu przyjmowaliśmy ustawę o kogeneracji, która dała wyższe o 20% ceny za energię uzyskiwaną z gazu importowanego z Rosji niż z gazu z biogazowni. O głos poprosił pan premier Mateusz Morawiecki. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dwa z waszej strony przeinaczenia i kłamstwa. Popatrzcie państwo, tutaj jest pierwsze, już przez was, przez pana posła przytoczone przed chwileczką.

Ale niestety pozbyliście się podstawowego atutu, jakim w 2008 r., bo w całym 2008 r. trwały negocjacje, i wcześniej. One były zaplanowane w taki sposób, żeby można było na koniec zawetować. I co powiedział premier Donald Tusk? Że nie będzie wetował. Szanowni państwo, jak ktoś na początku negocjacji mówi, że odkłada do szuflady swoje główne atuty, swoją bardzo skuteczną broń, to jaką pozycję negocjacyjną ma w całym procesie, który później następuje?

Prezydent Lech Kaczyński wiedział, jaka jest dynamika i logika negocjacji. Gdyby były to rządy Prawa i Sprawiedliwości, użyte byłoby to weto. Niestety nie skorzystaliście z tego.

Panie Marszałku! Panie Premierze! Panie Ministrze! Z wami nie da się normalnie pracować. Dzisiejszy dzień najlepiej obrazuje, jak PiS rządzi Polską.

Zachowujecie się tak, jakbyście parę dni przed świętami zostali zaskoczeni informacją, że od nowego roku czekają nas drastyczne podwyżki cen prądu. Tymczasem to, że podwyżki będą, było wiadomo wiele miesięcy wcześniej. Nie była to informacja zaskakująca ani nie wynikała z żadnych nagłych zmian w przepisach, ani nie jest efektem jakiejś nagłej katastrofy.

Nie wyszło i zamiast zajmować się rządzeniem krajem, tak naprawdę gasicie kolejny wizerunkowy pożar.

Rano wrzuciliście 12-stronicową autopoprawkę do nowelizacji, która miała 2 strony. Chcecie w ciągu godziny przepchnąć kolanem ustawę, która będzie decydowała o dystrybuowaniu miliardów złotych rokrocznie. Ale wracając do istoty problemu: Obiecaliście Polakom niezależność energetyczną, czyste powietrze, dobrobyt i świetlaną przyszłość naszej rodzimej gospodarki. A co mamy w zamian? Miliony ton węgla z Rosji, szokowy wręcz wzrost cen energii, smog i Polaków, którzy coraz częściej łapią się za własne portfele, zastanawiając się, gdzie znikają ich pieniądze. Co proponujecie? To oczywiście w jakimś niewielkim stopniu zniweluje podwyżki cen prądu, ale problemu nie rozwiąże. Co jeszcze proponujecie? Obniżenie opłaty przejściowej. W zasadzie to, co teraz proponujecie, to przecież wycofanie się z podwyżek wprowadzonych waszymi głosami w roku 2016 plus jakaś tam nadpłata, jeżeli chodzi o przedsiębiorców i odbiorców. Inną kwestią jest jednak pytanie, czy to faktycznie cokolwiek da. Opłata przejściowa to przecież odrębny podatek, który płacimy wraz z rachunkiem za prąd, tyle że ta opłata nie trafia do budżetu państwa, tylko gdzie, panie premierze? Do elektrowni węglowych. Jest pan ponoć ekonomistą, więc dobrze pan wie, że ta opłata została wprowadzona, by elektrownie węglowe miały pieniądze na niezbędne inwestycje. Zgadza się, panie ministrze? Zgadza się.

Więc co trzeba będzie zrobić? Czyli co trzeba będzie zrobić? Jeszcze raz podnieść opłaty za prąd, bo będzie znowu brakowało.

Prawo unijne zobowiązuje nas, by 50% dochodu ze sprzedaży uprawnień do emisji przeznaczyć na inwestycje nakierowane na ochronę klimatu. A co chce zrobić dzisiaj rząd PiS? 80% tych pieniędzy po prostu przejeść, dosypując je do spółek dystrybuujących prąd pochodzący głównie z węgla. To ma być transformacja energetyczna według PiS? Nie. Co z prawdziwą transformacją energetyczną w naszym kraju? Bez tego, bez długofalowych rozwiązań ceny energii będą dalej rosły, a szacuje się, że ta spirala będzie nakręcać się aż do 2030 r. Szanowni Państwo!

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. O tym, że drastyczne podwyżki cen prądu w 2019 r. są nieuniknione, mówiono od dawna. Przedstawiciele dzisiejszej, jak sami się nazwali, totalnej opozycji wielokrotnie używali tego argumentu, próbując dowieść, że obecny rząd jest nieudolny i nie radzi sobie z rządzeniem. Pomijali jednak fakt, że zapowiadane podwyżki nie są efektem ostatnich 3 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. że są skutkiem wieloletnich zaniedbań i zaniechań poprzedniej ekipy, słabo dbającej o polską gospodarkę i wyprzedającej wszystko, co miało wartość, nie tylko najlepsze polskie zakłady. Wystarczy zacytować wypowiedź przedstawiciela ówczesnej władzy Bartłomieja Sienkiewicza podsumowującego określeniem „kamieni kupa” dziedzictwo, jakie zostawiają. Nie dziwmy się więc, że naprawa Polski wymaga jeszcze długiego czasu. Nie zliczę ilości artykułów czy wywiadów, w których to premier Mateusz Morawiecki czy też jego ministrowie zapewniali, że pracują nad rozwiązaniem, które ochroni Polaków przed skutkami długotrwale źle prowadzonej polityki klimatycznej.

Można punktować, że jest to rozwiązanie tymczasowe, że nie rozwiązuje to problemów w sposób kompleksowy. Nie ma co ukrywać: tak właśnie jest.

Cieszy mnie, że rząd Zjednoczonej Prawicy już wiele razy pokazał, że dotrzymuje danego słowa: czy to przez realizację swoich obietnic wyborczych, czy też innych obietnic, jak w przypadku szkolnej wyprawki i programu Dostępność+, czy też dzisiaj - przez proponowanie rozwiązań nadzwyczajnych. Widać, że obecnie rządzącym zależy na swoich obywatelach i na polskich rodzinach. Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za dalszym procedowaniem nad tym projektem. Teraz głos zabierze pan poseł Ryszard Petru w imieniu koła Teraz! Wysoka Izbo! Dzisiejsza debata obnaża słabość całego państwa. Świadczy o braku wyobraźni, tchórzostwie i braku odpowiedzialności kolejnych rządów. I świadczy o ucieczce od problemów i o tym, że nie umiecie ich rozwiązywać. 9 mld w przyszłorocznym budżecie to koszt nieudacznictwa waszych rządów tylko w zakresie samej energetyki, a tak samo jest w innych branżach. Sami piszecie, że jest tylko na 1 rok, czyli przesuwacie podwyżki, drastyczne podwyżki prądu dla Polaków na czas tuż po wyborach. To nie jest żadne rozwiązanie systemowe, to jest rozwiązanie wyborcze. Ale proszę państwa, stan polskiego państwa w kontekście energetyki jest po prostu smutny. Od reformy górnictwa Janusza Steinhoffa za rządów Jerzego Buzka nie wydarzyło się w tej sprawie po prostu nic. Niestety tak było za SLD, tak było za Platformy i tak jest dzisiaj, za PiS-u. Ja tylko chciałbym zacytować kilka wypowiedzi z ostatnich lat, które pokazują, jak podlizywaliście się górnikom i jak ich oszukiwaliście: Górnictwo ma przed sobą wielką przyszłość i będzie się rozwijać. Prawie 90% energii uzyskujemy z węgla, a więc jeszcze przez długie lata będzie podstawą naszego bezpieczeństwa energetycznego. To oznacza, że górnictwo ma przed sobą wielką przyszłość i będzie się rozwijać. Obiecuję wam to. W naszym interesie jest, żeby węgiel nie stał się przeżytkiem. Węgiel to nasze czarne złoto, a Górny Śląsk i Zagłębie mogą być wielką perłą i świecić wspaniałym blaskiem na całą gospodarkę. Słuchajcie, Krzysztof Tchórzewski, minister energii: Państwo górnicy, więcej węgla nam potrzeba. Pomyślmy o tym, gdzie na Śląsku pobudować nową kopalnię. To pan premier Morawiecki, pan Tchórzewski jeżdżą po akademiach z okazji Barbórki, ale nie chodzą na pogrzeby ludzi, którzy umierają z powodu smogu. Nie widuje się ich w szpitalach, gdzie liczbę chorych z powodu smogu trudno nawet określić.

W ciągu ostatnich 2 lat polska energetyka bazowała na węglu. Dzisiaj 80% energii pochodzi z tego źródła. Weźmy dla porównania Niemcy.

Każdy odpowiedzialny rząd powinien natychmiast rozpocząć odchodzenie od węgla jako głównego źródła energii. Trzeba jak najszybciej wstrzymać - pan, panie premierze, dobrze to wie - wszelkie inwestycje węglowe, czyli budowę nowych bloków energetycznych, nie wspominając o chorym pomyśle budowy nowych kopalni. Odejście od węgla musi wiązać się również z postawieniem na odnawialne źródła energii. Pamiętajcie państwo: to wy, rządy PiS, zlikwidowaliście polską energię wiatrową. Musimy odejść od centralistycznego myślenia o energii. Kluczem ma być postawienie na lokalne źródła energii.

Inaczej się zatrujemy i będziemy mieć najdroższą energię w Europie. Nie ma tego w tym programie. Rozwój energetyki rozproszonej, promocja prosumentów, czyli samodzielnego wytwarzania energii przez konsumentów.

Kto dzisiaj eksportuje nowoczesne technologie związane z OZE? Ci, którzy na to stawiają, a my za miliardy będziemy tę technologię musieli kupować.

To jest po prostu humbug. Pan poseł Jakub Kulesza, Koło Poselskie Wolność i Skuteczni. Dziękuję. Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo!

I dzisiejszy kryzys energetyczny nie jest kryzysem. Jest skutkiem państwa interwencjonistycznej, państwa etatystycznej, państwa popisowej, państwa cały czas nieudolnej, centralnie sterowanej polityki. Mamy cztery duże spółki Skarbu Państwa, które zajmują się energetyką. Dlaczego cztery? Żeby zachować pozory konkurencji. Natomiast co to jest za konkurencja, jeżeli właścicielem wszystkich spółek jest jeden i ten sam podmiot - Skarb Państwa, i jest jeden i ten sam model zarządzania - z klucza politycznego. Jedyne pole, na którym te spółki Skarbu Państwa mogą ze sobą efektywnie konkurować, to jest załatwianie ciepłych posadek dla państwa, państwa rodzin, państwa dzieci, państwa znajomych. Jest to konkurowanie w załatwianiu, finansowaniu kolejnych państwa zabawek, takich jak Polska Fundacja Narodowa, i wyciągania z tych spółek - wydawałoby się - nieograniczonych źródełek. Śp. Stefan Kisielewski mawiał też, że socjalizm to jest ustrój, w którym bohatersko rozwiązuje się problemy nieznane w żadnych innych ustrojach. Ale z drugiej strony Ronald Reagan powiedział, że rząd nie jest w stanie rozwiązać żadnego problemu, bo to rząd sam te problemy tworzy. I prawda jest taka, jeżeli popatrzymy na dzisiejsze ceny energii, popatrzymy, co wpłynęło na ich wzrost, że będą to właśnie działania państwa, czyli polityków. Już był wspominany śp. Lech Kaczyński, który wracając z negocjacji pakietu energetyczno-klimatycznego, przyznał się, że zgodził się na założenia polityki bardzo ryzykownej dla Polski, ale to był gest względem pani Angeli Merkel. I to jest dla mnie zdrada interesu narodowego, że poświęca się naszą gospodarkę, nasze pieniądze - bardzo krótkowzrocznie - na rzecz innych państw, innych stolic. Jeżeli spojrzymy na ten pakiet energetyczny, na to, co ma on przynieść, do czego ma nas zmusić, to do głowy przychodzi mi tylko jeden cel: wspieranie niemieckiej gospodarki, niemieckiego przemysłu, który nastawił się na wdrażanie energetyki odnawialnej, wiatrowej, solarów słonecznych, paneli słonecznych. I państwo zastraszeni tą wielką emisją dwutlenku węgla, z czego Polska odpowiada za malutki procent całej emisji światowej, poświęcają nasz interes narodowy. Trzy wulkany spośród 800, które emitują dwutlenek węgla, emitują więcej tego dwutlenku niż cała polska gospodarka. Jakie jest rozwiązanie? Dużo było mówione o energetyce atomowej.

Jedyne, co ta spółka zrobiła przez 8 lat, to wydała miliony złotych na pensje: na ponad 34 tys. miesięcznej pensji prezesa, na 2 mln rocznie pensji dla zarządu, na 12 mln pensji dla zatrudnionych tam osób. W 2017 r. ta spółka miała przedstawić raport, miała przedstawić plan wdrażania energetyki atomowej. Nic państwo z tym nie zrobiliście. To kolejny przykład, jak państwowe pieniądze w łatwy sposób się wydaje. I my wszyscy jako obywatele odczuwamy tego skutki we własnych kieszeniach. Jeżeli państwo nie podejmą kroków w celu wycofania się z zapisów pakietu energetycznego, to ta obniżka akcyzy na nic się nie zda. Ten sam problem będziemy mieli za rok, za 2 i za 3 lata. Pan poseł Jan Klawiter, poseł niezależny. Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo!

I tutaj pierwsza sprawa, trzeba.

Potwierdziły to nawet agendy ONZ-owskie, które widząc potworne problemy z obroną klimatu, stwierdziły, że energetyka jądrowa musi być rozwijana. To jest ponad wszelką wątpliwość. Jest to zeroemisyjna energetyka, jest to niska cena energii. Starczy powiedzieć, że we Francji, która ma 70% energii jądrowej, cena energii jest dwukrotnie niższa niż w Niemczech, gdzie jest 13% udziału energetyki jądrowej.

Tak że przy 60 dniach, które w Europie często są praktycznie z niewielkim wiatrem, gdzie energia odnawialna dostarcza tylko 10% swoich, że tak powiem, możliwości, to musi być uzupełniane przez inne systemy, m.in. gazowy. Tak że muszą być i energia odnawialna, i atom. Bezwzględnie musimy iść w tym kierunku, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne. Jest jeszcze jedna uwaga.

Nie ma natomiast uwzględnionych źródeł objętych dyrektywą MCP, czyli źródeł ciepła od 1 do 50 MW, a tych przecież w Polsce jest największa liczba. I trzeba zwrócić uwagę, żeby wszystkie źródła, również i te małe, mogły być objęte wsparciem przez system zielonych inwestycji, bo one są szczególnie w tych średnich i mniejszych miastach. Teraz w trybie sprostowania pan poseł Neumann. 1 minuta, panie pośle. Panie Marszałku! Panie Premierze! Pan nie zrozumiał mojej wypowiedzi albo nie zna pan sprawy.

W tym zakresie posiedzenie to miało charakter przełomowy. Nie kryję, że Polska dążyła wszelkimi siłami, żeby porozumienie zostało zawarte, bo nie była to sprawa łatwa. Dlaczego to poparliśmy, to rozwiązanie klimatyczne? Dlatego że - jak mówiłem na początku - Polsce bardzo zależało, żeby ten szczyt zakończył się sukcesem. Przyjęcie zasady niewiążącego charakteru pakietu klimatyczno-energetycznego byłoby porażką i kolejnym dowodem na niemoc Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie pośle.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Fakty i harmonogram tamtych negocjacji - to, co pan zacytował, panie przewodniczący, panie pośle, to jest grudzień 2007 r. Kiedy była zawarta ta umowa w ramach Rady Europejskiej? Czyli to, co ktoś powiedział w ramach procesu negocjacyjnego, to jest coś zupełnie innego. Ale nikt nie pozbywa się swojej podstawowej broni, broni atomowej, a wyście się tego pozbyli w 2008 r.

A to, co ktoś powiedział rok wcześniej, w kontekście dochodzenia do tego, budowy sojuszu, jest zupełnie inną sprawą. Pan prezydent Kaczyński powiedział to, wiedząc, że w arsenale instrumentów rządu, ówcześnie już rządu Donalda Tuska, jest właśnie możliwość weta, i ta możliwość nie została wykorzystana. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, do pytań zgłosiło się ponad 60 osób. Bardzo proszę, jako pierwsza pani poseł Agnieszka Pomaska, klub Platformy Obywatelskiej.

Panie i Panowie Posłowie! Syn posła Smolińskiego, córka posła Cymańskiego, brat redaktora Rachonia z TVP Info, radni PiS, m.in. Kacper Płażyński, współpracownicy pana posła Horały - gdzieś go tu widziałam na sali - panowie Bełbot, Felmet, jego asystenci. Nie wystarczy 30 sekund, nie wystarczyłoby i godziny. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, tu nie było pytania. Teraz bardzo proszę o pytania. Można w pół minuty zadać pytanie, a oświadczenie pan poseł może wygłosić po zakończeniu części zasadniczej obrad. Pan poseł Mieczysław Kasprzak, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Panie Premierze! Mam pytanie: Po co przygotowywaliście tę podwyżkę cen energii? Przecież to wyście przygotowali. Pan o tym wiedział. Nie wiedział pan? Druga rzecz. Po co podnosiliście opłatę przejściową rok temu? Protestowaliśmy. Po co to wszystko robicie?

Pytanie zadaje pan poseł Zbigniew Ajchler, klub Platformy Obywatelskiej. Panie Marszałku! Panie Premierze! Panie i Panowie Posłowie! Ustawa jest bardzo ważna - 8,1 mld zł.

Wysoka Izbo! Dokonania PiS w ciągu ostatnich 3 lat to utrwalanie czarnej energii i podwyżki podatków. To jak ceny energii mają nie rosnąć? Teraz państwo zachowujecie się jak socjaliści w socjalizmie, czyli bohatersko próbujecie walczyć z tymi problemami, które sami stworzyliście. Niestety te podwyżki mają charakter fundamentalny i z powodu błędnej polityki PiS-u Polacy i tak zapłacą więcej za energię, więc ta ustawa to jest tylko i wyłącznie kiełbasa wyborcza. Bardzo proszę o pytanie. Wysoka Izbo! Ta ustawa zwiastuje, że PiS oficjalnie wchodzi w kampanię wyborczą. Zapowiadane przez was rozwiązania są po prostu nieprzemyślane, bo są tylko na 2019 r. A co dalej? Czy wiecie, że to były najdroższe święta od wielu lat? To wszystko przez podwyżki, które na każdym kroku fundujecie Polakom. Pan poseł Marek Sowa, klub Platformy. Wysoka Izbo! Dzisiejsza dyskusja to podsumowanie skutków polityki energetycznej rządów PiS-u. Jaka to polityka?

Dzisiaj wszyscy płacimy za skutki nieudolnej polityki rządu PiS. Pan poseł Tomasz Nowak, klub Platformy Obywatelskiej. Oto szafa, a w szafie mnóstwo trupów, trupów, które są efektem waszych 3-letnich rządów. Pierwszy trup wypada z szafy. To są podwyżki cen energii. Za chwilę będzie kolejny: niedoinwestowane szpitale, za chwilę będzie rolnictwo, za chwilę będą pensje nauczycieli, pielęgniarek itd., itd. Panie Premierze! Pytanie jest o odpowiedzialność, o odpowiedzialne rządy i odpowiedzialne rozwiązanie. Pan poseł Krzysztof Gadowski, klub Platformy.

Wysoka Izbo! Panie Premierze! Kłamstwa, kasa i propaganda to atrybuty pana rządu. Mówi pan o wzroście cen.

Bardzo proszę, pan poseł Marcin Kierwiński, klub Platformy. Wysoka Izbo! Pan premier Morawiecki albo wprowadza Wysoką Izbę w błąd, albo celowo kłamie. Panie Premierze! To, co mówił pan przewodniczący Sławomir Neumann w swoim pierwszym wystąpieniu, to był cytat z Lecha Kaczyńskiego z 2008 r. To wtedy Lech Kaczyński powiedział, że zgodził się na ryzykowną politykę klimatyczną, bo poszedł na rękę Angeli Merkel. Pani marszałek Barbara Dolniak, klub Nowoczesna. Panie Premierze! Proszę nam powiedzieć, jak to jest możliwe, że projekt ustawy liczy zaledwie 2 strony, a autopoprawka 12 stron, jak to jest możliwe, że przygotowaliście państwo projekt. w którym nie ujęliście tylu zagadnień natury prawnej, również z innych ustaw. To dowodzi tylko jednego. Nie macie państwo przygotowanych systemowych rozwiązań. Teraz pan poseł Paweł Pudłowski, klub Nowoczesna. Panie Premierze! Chciałem zapytać, czy sen energetyczny PiS-u trwa 3 lata. Nie zrobiliście nic, jeśli chodzi o kompleksowe rozwiązanie energetyczne. Dzisiaj co robimy? Ten stół tak czy inaczej się chybocze i te karteczki niestety nie pomogą.

Pan poseł Mirosław Pampuch, klub Nowoczesna. Pan poseł Jerzy Meysztowicz, klub Nowoczesna. Panie Marszałku Sejmu Niemego! Wysoka Izbo!

Pani poseł Paulina Hennig-Kloska, klub Nowoczesna. Panie pośle, pajacować to może pan gdzie indziej, a nie w Sejmie. Bardzo proszę. Proszę zająć miejsce.

Nie da się ukryć, że takie potraktowanie posłów Rzeczypospolitej Polskiej to jest po prostu kpienie z całego systemu demokracji w naszym kraju. Ale chciałam zapytać o niezwykle ważną rzecz: Czy ktokolwiek zbadał, czy autopoprawka nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej?

Wysoka Izbo! Panie Premierze! Chciałem się dowiedzieć, na jakim etapie są prace związane z budową elektrowni jądrowej w Polsce. Pytam w imieniu mieszkańców gmin Krokowa, Choczewo i Gniewino. Bardzo dziękuję, panie pośle. Panie Marszałku! Olsztyn - grupa zakupowa. To tylko przykłady. W jakim trybie mają zawrzeć nowe umowy? Pani poseł Ewa Lieder, klub Nowoczesna. Panie Premierze! Jak chcecie sfinansować inwestycje w OZE, skoro dzisiaj kilka miliardów poszło do pieca i na przejedzenie, czyli na spółki energetyczne? Miały pójść na zieloną, czystą energię. Pani poseł Krystyna Skowrońska, klub Platformy Obywatelskiej. Szybko panu poszło ze wzrostem VAT-u, 8 mld zł z kieszeni Polaków, ale długo pan odpowiada na list prezydenta Rzeszowa. Pan prezydent Rzeszowa czeka na odpowiedź.

Panie premierze, tak liczą samorządy. Pani poseł, nie zadała pani pytania. Dziękuję bardzo.

Chciałbym zapytać, dlaczego pan premier jest premierem wybiórczym, bo dane, którymi się pan posługiwał, były danymi wybiórczymi, które pasują do tezy, którą pan prezentuje. Zachowanie urzędnika państwowego, prezesa URE potwierdza, że polska gospodarka w sferze energetyki jest gospodarką sterowaną. Kombinowaliście z cenami na giełdzie, bo one wzrosły.

Panie Marszałku! Chciałabym zapytać, co zrobiliście z tymi miliardami z opłaty przejściowej, którą podnieśliście w 2016 r. Jakie to są instrumenty? To jest tajemnica handlowa, jak pan minister mi odpowiedział. Bo one zostały wyciągnięte z kieszeni Polaków.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Odkąd zaczął pan konkurować z prezydentem w wymyślaniu najmniej prawdopodobnych opowieści na temat pokładów węgla w Polsce, Polacy mają prawo do niepokoju. I tu w imieniu wyborców chciałbym zapytać: Czy prawdą jest, że ta ustawa jest oszustwem wyborczym tylko na ten rok? Czy wskutek tej ustawy zdrożeją: woda, chleb, paliwo, bilety kolejowe i wywóz śmieci? Pani poseł Zofia Czernow, klub Platformy Obywatelskiej. Panie Premierze! Mam pytanie: Co dalej z podwyżkami cen energii dla samorządów, w przypadku których ceny te wzrosły nawet o 80%? Czy te podwyżki zostaną cofnięte? I drugie pytanie: Jakie skutki dla projektu budżetu państwa na 2019 r. wywoła ten projekt ustawy? Bardzo dziękuję. Pani poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, klub Platformy Obywatelskiej. Wysoka Izbo! Mam 30 sekund, więc jedno bardzo krótkie pytanie: Kiedy przestanie pan zaklinać rzeczywistość i zacznie naprawdę troszczyć się o codzienność, o bezpieczną codzienność naszych obywateli, tylko tak prawdziwie, a nie z doskoku i w ostatnim dniu roku? Pani poseł Joanna Frydrych, klub Platformy Obywatelskiej. W uzasadnieniu projektu czytamy, że ustawa ma zapobiec skokowej podwyżce cen energii w 2019 r. A ja pytam: Co w 2020 r. i w kolejnych latach? Czy taki zapis nie jest formą szantażu politycznego?

Wysoka Izbo! Myślę, że niepotrzebnie macie pretensje do pana Terleckiego, marszałka, jeżeli chodzi o te 30 sekund. To jest wizjoner, to jest wielki wizjoner, proszę państwa.

Wysoka Izbo! Problem nie polega na tym, że decydujemy o VAT, o opłatach przejściowych, które zostały po prostu podniesione wcześniej, ale na tym, że nie bierzemy pod uwagę bardzo ważnej rzeczy, która stanowi kilkadziesiąt procent wartości energii elektrycznej. W jaki sposób utrzymacie tą cenę surowca?

Wysoka Izbo! Chcecie zahamować te podwyżki, bo boicie się, że przegracie wybory, ale macie bardzo dobre przeczucie, bo tak będzie. W swojej wypowiedzi sugeruje pan, abyśmy pilnowali samorządowców. Mam pytanie: W jaki sposób będą renegocjowane umowy, które już zostały zawarte przez jednostki samorządu terytorialnego? Pan poseł Paweł Bańkowski, klub Platformy Obywatelskiej. Ceny energii w roku 2019 wzrosną. Proszę nie okłamywać Polaków.

I kolejne pytanie: Kiedy rozpoczną się renegocjacje dotyczące cen z samorządami i przedsiębiorcami, z którymi spółki energetyczne zawarły już umowy? Pan poseł Wojciech Król, klub Platformy Obywatelskiej. Ta ustawa to dowód na to, że myśli pan tylko i wyłącznie o wyborach parlamentarnych, a nie o kolejnych latach. Nie interesuje pana to, jakie rachunki zapłacą Polacy w 2020 r. Czy ma pan odwagę tutaj wyjść i powiedzieć Polakom, jakie rachunki zapłacą w 2020 r. Pani poseł Maria Janyska, klub Platformy Obywatelskiej. Panie Premierze! Dobrze się pan czuje w tym chaosie, w tym procederze legislacyjnym? Chyba tak, bo całe pana wystąpienie było chaotyczne i lekceważące. Pan pokazał tym wystąpieniem, że ani pan nie liczy, ani nie łapie wątków, ani nie ma pan klasy politycznej.

Pani poseł też nie udało się zadać pytania. Szanowni Państwo!

Każdy odpowiedzialny rząd myśli strategicznie, wiele lat do przodu, ale was interesuje tylko koniec własnego nosa, chyba że chodzi o zatrudnienie dzieci w spółkach energetycznych, o czym słusznie powiedziała moja koleżanka. Chciałam zapytać, czy dalej będziecie państwo bazować głównie na [[Dzwonek]] imporcie węgla. Pan poseł Grzegorz Furgo, klub Platformy Obywatelskiej. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Premierze! Pan się wywróci na tej ustawie, bo pan nie jest szczery w stosunku do Polaków. Chciałbym powiedzieć państwu jedną rzecz.

Dla pana premiera, jak za komuny, liczy się prawda ekranu, a ja powiem teraz o prawdzie czasu.

Pan poseł Michał Stasiński, klub Platformy Obywatelskiej. Wysoka Izbo! Propozycje struktury niektórych zmian w strukturze cen detalicznych oraz zasad rekompensaty skutków tych zmian.

Farsą było pana wystąpienie, panie premierze, farsą jest wasza polityka energetyczna i farsą jest forma tej debaty.

Panie Premierze! Już kiedyś panu mówiłam, że jest pan Pinokiem polskiej polityki, ale po dzisiejszej pana wypowiedzi mogę tylko tutaj w zasadzie powiedzieć, że Pinokio to jest przy panu pikuś.

W Toruniu oferty na zakup energii na 2019 r. są wyższe o 60%. Pan poseł Jakub Rutnicki, klub Platformy Obywatelskiej. Panie Marszałku!

Cały czas pan o tym zapomina. Warto o tym przypomnieć. Gmina Sieraków - wzrost cen o 63%. Panie premierze, czy pan wyśle pisma zapewniające, że te ceny są już nieaktualne i że te podmioty nie będą [[Dzwonek]] ponosić wyższych kosztów w 2019 r. dla miasta stołecznego Warszawy od nowego roku wzrosną o 67%. Ale, Wysoka Izbo, nie wszyscy przejmują się podwyżkami prądu. Czy Wysoka Izba wie, co to jest za liczba?

Mimo dużego wysiłku nie udało się panu zadać pytania. Bardzo proszę, pan poseł Ireneusz Raś, klub Platformy Obywatelskiej. Panie Premierze!

Pan reaguje dopiero dziś. Pan poseł Cezary Grabarczyk, klub Platformy Obywatelskiej. Panie Premierze! Jedyną osobą, która panu dziś uwierzyła, że prąd nie zdrożeje, jest prezes Jarosław Kaczyński. Pan poseł Włodzimierz Karpiński, klub Platformy Obywatelskiej.

Obniżacie państwo konkurencyjność polskiej gospodarki.

Przepraszam, panie pośle. Czy kontestowanie polityki klimatycznej Unii Europejskiej jest kolejną odsłoną pana proeuropejskości? Może rozpocząłby pan ponowne wprowadzanie Polaków do Europy, z czystym powietrzem, a nie w oparach smogu najgorszego w Europie? Z tym wiąże się kwestia tego, że ceny energii elektrycznej w Polsce są zależne od emisyjności polskiej gospodarki.

Wysoka Izbo! Jak to jest, że Polacy wydali setki złotych na energooszczędne żarówki, zużywające 10 razy mniej prądu, a płacą za prąd tyle samo? Jak to jest, że Polacy wydali tysiące złotych na coraz lepsze lodówki, pralki i co tylko można, z klasą A+++, więcej plusów, niż wy dajecie, a płacą za prąd tyle samo? Pan poseł Paweł Grabowski, klub Kukiz’15. Panie premierze, mówi pan, że nie będziemy grzebać w kieszeniach Polaków, nie będziemy tam wsadzać dłoni. Wobec tego mam pytanie: Kiedy wyciągniecie drugą dłoń, ponieważ człowiek ma dwie dłonie i fiskus ma też dwie dłonie? Jedną, jak mówicie, nie grzebiecie w kieszeni, a drugą wyciągacie ogromne kwoty. Kiedy w końcu państwo podwyższycie kwotę wolną od podatku, by Polaków było stać na to, żeby płacić takie rachunki, jakie chcą, za tyle, ile zużywają?

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wielokrotnie pan, panie premierze, mówił o reformie państwa. W związku z tym mam pytanie: Czy pana reformy polegają na tym, że minister środowiska w trosce o środowisko wycina drzewa, że minister energii w trosce o odnawialne źródła energii zwalcza wiatraki, a pan, wprowadzając nowoczesne rozwiązania w gospodarce, ściąga na potęgę węgiel z Rosji? Pan poseł Marek Suski, klub Prawo i Sprawiedliwość. Panie Premierze! Wysoka Izbo! Mam pytanie: Ile trzeba by sprowadzać węgla, gdyby zlikwidowano te kopalnie, które chciała likwidować Platforma Obywatelska? Ewa Kopacz i strzelanie do górników. Ile straciliśmy na opóźnieniu budowy gazoportu przez Platformę? Jeszcze jedna sprawa. Tutaj są absurdalne zarzuty. Wysoka Izbo! Pytanie, żeby nie było. Panie premierze, komu pan zabierze te 9 mld, żeby zrealizować zapisy tej ustawy? Pan poseł Antoni Mężydło, klub Platformy Obywatelskiej.

Panie Premierze!

Pan poseł Marcin Święcicki, klub Platformy Obywatelskiej. Panie Premierze! Wysoka Izbo! Od 2015 r. ceny energii elektrycznej w Europie spadają, a w Polsce ceny energii elektrycznej rosną. Europa idzie w kierunku energii taniej i czystej. My idziemy w kierunku energii brudnej i drogiej. Kiedy zmienimy ten trend? Wszystkie te wygibasy z opłatami spowodują, że może gospodarstwa domowe zapłacą mniej, ale my jako podatnicy zapłacimy więcej, bo koszty produkcji energii cały czas rosną. Panie Marszałku! Czy pan wie, że w 2010 r. ceny energii z fotowoltaiki zrównały się z cenami energii z elektrowni nuklearnych? Czy pan wie, że w 2018 r., w 100-lecie naszej niepodległości, na listopadowych aukcjach ceny energii z wiatru na lądzie okazały się niższe od cen energii na giełdzie towarowej?

Panie Premierze! Ceny węgla z polskich kopalni w roku 2017 wzrosły o ok. 25%, zaś import węgla z Rosji w pierwszych 9 miesiącach tego roku wzrósł o 72% w stosunku do roku 2017.

Panie premierze, trzeba było zwyczajnie w świecie sprawniej doradzać. Pan poseł Maciej Małecki, klub Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma pana posła.

Wysoki Sejmie!

Takie słowa w ogóle nie padły. Z tych przewidywań i analiz, które były tu podstawą, wynikało, że po pewnym czasie budowa wiatraków na lądzie przestanie się opłacać.

Jeśli chodzi o efektywność energetyczną wiatraków na morzu, te najnowsze dochodzą do 50% efektywności.

To jest naturalna tendencja, którą widać w innych państwach. Dlatego w tej chwili trwa budowa instalacji wiatrowych na lądzie i ostatnie aukcje wykazały pewne zainteresowanie, ale wcale nie takie olbrzymie. Mamy miejsca, gdzie można budować. Chcemy, żeby były tam budowane farmy fotowoltaiczne, które są w Polsce bardzo potrzebne ze względu na szczyty mocowe, szczyty zapotrzebowania na energię latem, które występują przy jednocześnie bardzo słonecznych dniach.

Chciałbym jednoznacznie sprostować - nie mamy zamiaru niczego sztucznie, na siłę, likwidować, niczego złomować.

Otóż mamy tego typu sytuację, że zapotrzebowanie na energię znacząco wzrosło i w dużym zakresie wzrosło wykorzystanie elektrowni - podstawowe elektrownie to są elektrownie węglowe - więc wzrosło ich wykorzystanie. Otóż po 2021 r. będzie zamykana znaczna część obecnie istniejących bloków energetycznych, tych najstarszych, z lat 60., 70., które nie będą się już finansowo kwalifikować do tego, żeby zainstalować w nich instalacje BAT-owskie związane z podniesieniem standardu emisyjnego. I tutaj jest kwestia taka, że zmniejszy się zużycie energii elektrycznej, będzie to nie mniej niż 6–7 GW.

Kilka lat możemy poimportować. Węgiel jest importowany w zależności od tego, jaki jest potrzebny.

Chodzi o tryb.

To jest tryb przyjęty w tym momencie, już zapisany szczegółowo w ustawie, w jaki sposób będą się te rozliczenia odbywały. A więc tutaj nie ma żadnych zagrożeń.

A więc w tej dziedzinie nie ma żadnych zagrożeń.

Chciałbym też podkreślić i nawiązać właśnie do tej pierwszej części naszej ustawy, jeżeli chcemy tak się do tego odnieść, bo państwo wielokrotnie podkreślaliście, że to jest na 2019 r. Spójrzmy do ustawy.

Żadna data nie jest wpisana. I już widzimy, że w tej dziedzinie nie będzie żadnej zmiany.

Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zawarty w drukach nr 3112 i 3112-A, do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Proponuję na podstawie art. 39 ust. 3 regulaminu Sejmu, aby Sejm wyznaczył termin przedstawienia sprawozdania umożliwiający rozpatrzenie go na bieżącym posiedzeniu Sejmu.

Ale wcześniej jeszcze proszę pana posła sekretarza o odczytanie komunikatów. Komunikat jest nieaktualny. Za 5 minut przystąpimy do głosowania.

Wznawiam obrady. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zgłoszono wniosek o skierowanie projektu ustawy dodatkowo do Komisji Gospodarki i Rozwoju. Propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu jest, aby Sejm skierował ten projekt ustawy do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał. Dokończę zdanie. że Sejm propozycję zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu przyjął, a wniosek o dodatkowe skierowanie tego projektu ustawy poddam pod głosowanie. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za dodatkowym skierowaniem projektu ustawy, zawartego w drukach nr 3112 i 3112-A, do Komisji Gospodarki i Rozwoju, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Proponuję na podstawie art. 39 ust. 3 regulaminu Sejmu, aby Sejm wyznaczył termin przedłożenia sprawozdania umożliwiający rozpatrzenie go na bieżącym posiedzeniu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę rozumiał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Proszę pana posła sekretarza o odczytanie komunikatu. Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji: do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Finansów Publicznych 15 minut po zakończeniu pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką, druki nr 3112 i 3112-A, w sali nr 118. Dziękuję. Zarządzam przerwę do

Wznawiam obrady. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 3113. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjął decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 3112, 3112-A i 3113) Proszę pana posła Macieja Małeckiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo!

W czasie posiedzenia zostały zgłoszone dwie poprawki, które komisje przyjęły i rekomendują Wysokiej Izbie. Komisje przyjęły ten projekt ustawy bez głosów sprzeciwu i rekomendują Wysokiej Izbie oczywiście przyjęcie projektu ustawy. Dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Maciej Małecki, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Przypomnę, że celem ustawy jest ochrona polskich rodzin, polskich firm, przemysłu i samorządów przed negatywnymi skutkami skokowego wzrostu cen energii elektrycznej, jaki obserwujemy w całej Polsce. Przyczyn wzrostu cen energii w Europie i w Polsce jest kilka, ale źródłem problemu horrendalnego wzrostu cen energii były złe decyzje z roku 2008. Tych decyzji nie zawetowali nasi poprzednicy i dziś musimy to naprawiać. Rząd wypracował mechanizm, który szerokim parasolem ochroni przed podwyżkami cen zarówno odbiorców domowych, jak i firmy i samorządy.

Jest to mechanizm z wizją na przyszłe lata, nie tylko na rok 2019, dlatego też warto ten mechanizm docenić. Nie jest to łatanie dziur, ale budowanie stabilnej przyszłości dla niskich cen energii w Polsce. Podsumowując: przyjmując tę ustawę, chronimy Polaków przed wzrostem cen energii elektrycznej. Potencjał tej ustawy dostrzegły już połączone komisje, Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisja Finansów Publicznych, które przyjęły ten projekt bez głosu sprzeciwu. Tym samym Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisja Finansów Publicznych dały Wysokiej Izbie zielone światło na przyjęcie tej ustawy, przyjmując ją, jak powiedziałem, bez głosu sprzeciwu. Jest to dobra okazja dla Wysokiej Izby do głosowania ponad podziałami. Zachęcam państwa do głosowania ukierunkowanego nie politycznie, ale troską o portfele Polaków.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z mojego punktu widzenia. Miałem możliwość obserwowania wielu premierów, ale to, co usłyszałem dzisiaj, było dla mnie bardzo wielkim zaskoczeniem. A dlaczego? Dlatego że mamy okres świąteczny, mamy próbę ratowania tego, do czego doprowadziła polityka tej opcji. Co usłyszeliśmy? Nie prośbę o współdziałanie. Nie prośbę o pochylenie się nad propozycjami, tylko atak na opozycję, na ludzi, którzy są winni tego, co są. Jak inaczej brzmi prośba posła sprawozdawcy, który mówi, że ma nadzieję, że te propozycje przyjmiemy. A dlaczego jestem zaskoczony postawą pana premiera?

My proponowaliśmy wprost zmniejszenie akcyzy. A co teraz jest proponowane? Fundusz, który może iść na wsparcie odnawialnej energetyki, fundusz, który może pójść na likwidację niskiej emisji, fundusz, który może pójść na wzrost efektywności, będzie skierowany na następną instytucję publiczną, na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Stworzy się administrację, która ten fundusz będzie dzielić i dawać wsparcie spółkom, które dyktują warunki na naszym rynku. Powinniście popatrzeć, bo za każdym z nas stoją obywatele. Zniszczenie rynku energii doprowadziło wprost do tego, że znaleźliśmy się w przededniu nowego roku w sytuacji bez wyjścia. Państwo też znaleźliście się w tej sytuacji. Deklaracje, że nie będzie wzrostu cen, to były puste deklaracje. Na naszym rynku stworzono w 2015 r. monopol wytwórcy energii i spółek paliwowych, który dyktuje ceny. Proszę przyjąć do wiadomości, państwo posłowie z tej strony sali, że nie ma konkurencji na rynku. Zlikwidowano obligo giełdowe. Zlikwidowano możliwość wyboru najtańszego odbiorcy, przepraszam: dostawcy. Doszliśmy do momentu, gdzie Wysoka Izba i również my, Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska, chcemy pomóc obywatelom. Bo nie może za nieudolność władzy płacić Bogu ducha winny obywatel. Ale deklaruję z tej pozycji, że od 2 stycznia będziemy składać propozycje zmian ustawowych. Będziemy patrzeć na ręce. Niech mi ktoś z państwa posłów powie. Bo tu jest tylko polityka. Powiedzcie mi państwo posłowie, w którym miejscu ta ustawa obniża koszty wytwarzania energii elektrycznej? W którym miejscu? Nie ma nic o ograniczeniu kosztów. Spółki państwowe będą miały to, co będą chciały, a płacił będzie, bez względu na wszystko, odbiorca końcowy, czyli obywatel. Szanowna Pani Marszałek! Dajemy też szansę wyjścia naprzeciw temu, co powiedziałem, odtworzeniu rynku energii. Zgłaszam dwie poprawki.

Proszę o zabranie głosu pana posła Józefa Brynkusa, klub Kukiz’15. Wysoka Izbo!

To jest przelewanie z pustego w próżne. Przez 3 lata rządów PiS, a wcześniej PO-PSL. Podam konkretne przykłady. Jest elektrownia wodna zbudowana na zaporze Świnna Poręba na Jeziorze Mucharskim.

Dwa razy była szumnie otwierana: raz przez przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, a potem przez panią premier Beatę Szydło. Produkuje? Nie produkuje energii elektrycznej. Urządzenia są warte kilkadziesiąt milionów złotych. Jeżeli 9 mld ma kosztować ta zmiana, którą chcemy teraz wprowadzić, to te kilkadziesiąt milionów złotych też byłoby istotną wartością.

Następna sprawa. Za tym należy się opowiedzieć. W cenie energii elektrycznej najważniejszą rzeczą to jest koszt surowca. Problem polega na tym, że w Polsce podstawowym surowcem jest węgiel, w przypadku którego jest kilkadziesiąt opłat różnego rodzaju, począwszy od akcyzy, skończywszy na opłatach środowiskowych. To jest główne pole do obniżki cen energii elektrycznej. To rząd powinien zaproponować, wiedząc, że od 2019 r. ceny energii muszą wzrosnąć, a nie wprowadzać rozwiązań w totalnym chaosie prawnym, ekonomicznym i społecznym. Strach, jak widać, ogarnął także rządzących i powstała kolejna proteza legislacyjna. Jakoś nikt z rządzących nie zająknął się, że ta proteza będzie obowiązywać krótki czas, że jest to rozwiązanie tymczasowe. Deklaracje, które państwo tutaj wygłaszacie, że coś nie wzrośnie, już na tej sali wielokrotnie słyszeliśmy. Pani premier Beata Szydło przy okazji debaty nad Prawem wodnym mówiła w ten sposób: nie wzrosną ceny wody i ścieków. To jest nieprawda. Wystarczy, że spyta o to w tej gminie, w której jest mieszkanką, i inne jednostki samorządu terytorialnego. Ceny wody i ścieków wzrosły. I na koniec: nie bójcie się przyznać, proszę państwa, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, że propozycje, o których mówił wcześniej marszałek Tyszka, które składaliśmy w formie ustawy, służą Polsce i Polakom. Weźcie nasze rozwiązania w całości, a nie tylko fragmentarycznie. Jeżeli już obniżacie VAT i akcyzę, to do stawek minimalnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Zrezygnujcie z tego Bizancjum, które panuje w spółkach Skarbu Państwa.

Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Cóż, rządzący zafundowali Polakom podwyżkę cen energii elektrycznej, a dzisiaj szukają winnych. Wiedzieliście, co się dzieje, jaka jest cena węgla, jaka jest cena uprawnień do emisji. Nie było żadnej reakcji. Minister na jednym z posiedzeń mówił wprost: samorządom nieźle się powodzi, mają wyższe dochody, jakoś sobie poradzą. Takie było stanowisko. Polacy też sobie poradzą, bo daliśmy pieniądze, 22 mld, jakoś to zniosą.

To jest bardzo zła ustawa. Jej się nie da wprowadzić w życie. I jak dzisiaj, panie pośle sprawozdawco, cieszyć się, że wszyscy to poparli? Mieliśmy podpisać się pod tym, że Polacy dostaną 80-procentowy wzrost cen energii? Poparliśmy to, ale to jest niewykonalne. Psujecie system energetyczny.

Ceny energii wzrosną. Kiedy samorządy mogą zacząć kalkulować nowe ceny energii? W marcu, w kwietniu? System energetyczny, który powinien być spójny, który nie może być regulowany z dnia na dzień, w tym momencie nam się sypie. To będzie nie do opanowania.

Przecież rok temu podnieśliście o 50%.

My zgłosimy kilka poprawek, które może w jakiś sposób ucywilizują ten zły projekt. To jest projekt, który ma dać sygnał obywatelom, Polakom, jak to wspaniale naprawiacie błędy

Jedna z naszych poprawek idzie w kierunku zmniejszenia VAT-u na energię odnawialną.

Odrzuciliście to. Wszystkie wasze działania, zaniechania w zakresie energii odnawialnej dzisiaj mają odzwierciedlenie w cenach emisji. Więc to też jest przykład, jak przez 3 lata można zepsuć cały system.

Panie i Panowie Posłowie! Mydlicie Polakom oczy, mówiąc o repolonizacji i wstawaniu z kolan, ale mówiąc „polskie”, myślicie „państwowe”, myślicie „nasze, gdzie nasi ludzie usiądą i będą mogli się obłowić” Mówiąc o wolności gospodarczej, wprowadzacie ceny regulowane rodem z epoki Gierka. Gospodarkę centralnie sterowaną raz już przerabialiśmy. Pozostały nam po niej długi, pustki w kasie i hiperinflacja. Zamiast zwracać uwagę na rachunek ekonomiczny, upolityczniacie decyzję w obrębie spółek energetycznych. Szukanie kozła ofiarnego nic tu nie da.

To, co proponujecie w ramach złożonej autopoprawki, może okazać się niedozwoloną pomocą publiczną. Wielu ekspertów wprost wskazuje, że to po prostu jest pomoc publiczna, którą zakwestionuje Unia Europejska, bo to są dopłaty do stałych taryf energii, po prostu transfer środków do zintegrowanej energetyki węglowej. Zamiast rozwijać OZE, będziemy dopłacać do węgla przez kolejne lata. Przecież prezydent zapowiedział - 200 lat. Natomiast jest pytanie, na które pan minister dzisiaj nie raczył odpowiedzieć, bo odpowiedzi nie zna. Co się stanie, jeśli Komisja Europejska faktycznie zakwestionuje te rozwiązania i uzna je za niedozwoloną pomoc publiczną? Będziemy musieli zabrać te pieniądze ze spółek energetycznych i nie będziemy mogli tego uzupełnić z budżetu państwa, bo to też będzie niedozwolona pomoc publiczna. Cała ta dyskusja, która dzisiaj toczyła się w komisji, miała nam dać odpowiedź na jedno podstawowe pytanie - czy skazujecie Polaków dzisiaj na podwójne koszty, na pokrycie tego, co trzeba będzie oddać w ramach niedozwolonej pomocy publicznej, i na kary, które zostaną nałożone przez Komisję Europejską na Polskę. Pytaliśmy, gdzie jest opinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie notyfikacja Komisji Europejskiej, skoro wchodzimy w obszary, które rodzą tego typu wątpliwości. Nie ma. Potraficie tylko teoretycznie siedzieć na stołkach i udawać, że cokolwiek robicie. Już wiele razy słyszeliśmy, że jest okej, a potem gasiliście międzynarodowe afery, jak miało to miejsce w przypadku ustawy o IPN, wzniecone niepotrzebnie międzynarodowe wielkie kryzysy, wycofywaliście się z rozwiązań, które były dla was zgodne z prawem unijnym, zgodne z konstytucją, tak jak w przypadku Sądu Najwyższego czy chociażby podatku handlowego. Wiele razy mówiliście, że wszystko jest okej, a potem okazywało się zupełnie co innego.

Ale, co najważniejsze, pojawiają się wątpliwości, co z tymi samorządami, które podpisały nowe umowy na podstawie wcześniej rozstrzygniętych przetargów. Ustawa wprost tego nie mówi.

Natomiast na regulowane ceny i PRL-bis zgody z naszej strony nie ma.

Bardzo dziękuję.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Gmeraliście już przy wielu sprawach państwa, ale dopiero jak włożyliście łapy w energetykę, to was poraziło. To wasze pierwsze spotkanie z prawdziwymi problemami. Podwyżka cen prądu dopiero przed nami.

Zaskoczyły was podwyżki prądu i zamiast rozwiązać problem, przesuwacie go w czasie. Przed nami jest bardzo trudny rok.

Jeżeli tak będzie, to budżetu na rok przyszły nie można kreować w sposób nonszalancki. W tym roku koszty wytworzonej energii odnawialnej w Polsce z wiatru czy z fotowoltaiki są niższe niż z węgla. A to oznacza, że ci, którzy stawiają na energię odnawialną, tak naprawdę stawiają na energię czystą i tanią. W zeszłym roku w Australii zbudowano po raz pierwszy kosztem 90 mln dolarów pierwsze bloki do przechowywania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a w tym czasie PiS lekką ręką wywala 9 mld zł z budżetu po to, aby w okresie wyborczym uniknąć uderzenia w portfele Polaków. Ale macie 9 mld, żeby utrzymać własne stołki, dobrze wiecie, że podwyżki będą jeszcze wyższe - po wyborach. Decyzja o zakończeniu wydobycia surowca w Niemczech zapadła w 2007 r. A w perspektywie 4 lat zostaną tam jeszcze zamknięte wszystkie elektrownie jądrowe. Dobrze by było, gdybyście państwo z PiS-u wzięli długopisy i zapisali. Panie ministrze, czy pan je zna?

Polska będzie zmuszona kupować energię odnawialną z innych krajów europejskich. Do tego doprowadziła wasza polityka. Koszt takiego zakupu rocznie to jest ponad 8 mld zł. Skazujecie Polskę na to, abyśmy kupowali z zagranicy energię odnawialną, żebyśmy importowali węgiel z Rosji, żebyśmy truli Polaków i jeszcze musieli dopłacać do tego, żeby ceny nie rosły. Oznacza tak naprawdę to, że uzależniamy się od biorców zewnętrznych. Proszę państwa, mam do państwa pytania, do pana premiera, pana ministra. Jak przekona pan Komisję Europejską, że ustawa ta nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej? Panie ministrze, czy można od pana uzyskać tę odpowiedź?

Przypomnę, że jeżeli będzie to pomoc publiczna, to pieniądze trzeba będzie po prostu wycofać. Kto za to będzie płacił? Kolejne rządy, ale kolejne rządy są. To są pieniądze nas wszystkich. Proszę państwa, będziemy głosować przeciwko tej ustawie.

Pan poseł Jacek Wilk, Wolni i Skuteczni. Bardzo dziękuję. Panie i Panowie Posłowie! Wysoka Izba nas przyzwyczaiła do tego, że prowadzimy tu mnóstwo absurdalnych dyskusji, dlatego zacznę od cytatu. W czasie burzy babcia stawiała w oknie święty obraz, aby piorun trafił w obraz, a nie w dom. Ten cytat z zeszytów szkolnych bardzo dobrze oddaje absurd tego, co tu się dzieje. Oczywiście absurdem pierwotnym jest tzw. pakiet klimatyczny. Warto sobie uświadomić, skąd się biorą takie pomysły. Lewica nigdy nie wierzyła w to, że można uzyskać dobrobyt dzięki pracy, produkcji, przemysłowi, a najlepszym sposobem jest grabież i rabunek. Dlatego zawsze wymyślano różne rewolucje albo wojny, za pomocą których ograbiano właśnie tych, którzy jakiś majątek posiadali. Teraz prowadzenie wojen i różnych rewolucji jest niemodne, przynajmniej oficjalnie, bo się prowadzi różne misje stabilizacyjne, akcje pokojowe, akcje humanitarne, które są wojnami, tylko bez wypowiedzenia wojny. Zamiast tego toczy się wojnę z klimatem. Szanowni Państwo! Wojna przeciwko klimatowi ma oczywiście taki sam sens jak różnego rodzaju zabobony, które przez całe wieki się pojawiały. Natomiast tzw. badania naukowe mają potwierdzać zasadność zmian klimatu spowodowanych tzw. globalnym ociepleniem. Oczywiście teorie naukowe podrzucają różne ciekawe koncepcje, np. takie, że bydło produkuje za dużo gazów cieplarnianych. No cóż, naukowcy to ludzie praktyczni i wychodzą z założenia, że głupio jest płacić za takie badania, ale jeszcze głupiej jest pieniędzy za to nie brać. Pytanie tylko, dlaczego my akurat mamy na tym wszystkim bazować. Są to, tak jak powiedziałem, takie same zabobony jak kiedyś, tylko oparte nie na wierzeniach, a ideologii. Notabene jakiś czas temu agencja kosmiczna NASA podała informację, że stopieniu ulegają pierścienie Saturna. Odpowiedź ekologiczna, że na Saturnie jest za dużo kopalni i elektrowni węglowych i za dużo krów, które produkują gazy cieplarniane. Albo odpowiedź zdroworozsądkowa, że zmiany te wynikają po prostu z aktywności Słońca. Ale rozumiem, że oczywiście ta przez Unię Europejską nie jest brana pod uwagę. Ludzie wierzą w różne rzeczy: w yeti, w UFO. Ostatnio zapłaciliśmy np. 250 mln zł za zlot wyznawców religii globalnego ocieplenia. Szanowni Państwo! Mógłbym zalecić oczywiście rządowi, aby poszedł po zdrowy rozsądek i po prostu pakiet klimatyczny wypowiedział. Ale nie sądzę, żeby rząd to zrobił, ponieważ zawsze ulega Unii Europejskiej. Wobec tego tak jak Zagłoba poradzę rządowi, aby pił więcej wina, ponieważ, jak mówił Zagłoba: Picie wina powoduje, że oleum unosi się do głowy. Szanowni Państwo! Oczywiście każda obniżka akcyzy jest korzystna i my to poprzemy, tylko warto sobie wyjaśnić, na czym polega akcyza. Przecież prąd to wielki luksus, można by się obejść bez niego, siedzieć przy świeczkach, może nawet więcej dzieci by się dzięki temu urodziło.

Z tego powodu, szanowni państwo, jestem stanowczym przeciwnikiem tego typu polityki i uważam, że Unia Europejska powinna być zniszczona. Bardzo dziękuję. Teraz głos zabierze pan poseł Piotr Liroy-Marzec. Wysoka Izbo! Panie Premierze! Sezon na wycofywanie uważam za otwarty. Niedawno Platforma Obywatelska wycofała się z wycofania bonifikaty na użytkowanie wieczne w Warszawie. teraz pan premier wycofuje się z podwyżki cen prądu. Pan premier wycofuje się z podwyżki cen prądu i proponuje w tym projekcie ustawy obniżkę podwyżki. Obniżka podwyżki jest jedynym wyjściem, ponieważ rząd PiS kontynuuje politykę rządu PO. Jako przewodniczący koła Wolność i Skuteczni będę głosował za przedstawionym projektem ustawy. Jako prezes Skutecznych będę przyglądał się, czy po wyborach rząd nie wycofa się z obniżki podwyżki. Bardzo dziękuję.

Panie Marszałku! Wnoszę o natychmiastowe przejście do trzeciego czytania bez odsyłania ustawy do komisji po dostarczeniu poprawek.

W dyskusji zgłoszono wniosek o przystąpienie do głosowania nad tym projektem ustawy po doręczeniu zestawienia poprawek. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Słyszę sprzeciw.

Wznawiam obrady. Kontynuujemy rozpatrywanie punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W dyskusji zgłoszono wniosek o niezwłoczne przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy po doręczeniu zestawienia poprawek, bez odsyłania do komisji. Wobec zgłoszonego sprzeciwu poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem wniosku o niezwłoczne przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy po doręczeniu poprawek, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek przyjął. Przystępujemy do trzeciego czytania. Zestawienie zgłoszonych poprawek zostało państwu doręczone do druku nr 3113. Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 2. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 1. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Kto z państwa jest za przyjęciem 3. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Kto z państwa jest za przyjęciem 5. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. W 6. poprawce wnioskodawcy proponują skreślić art. 3 projektu ustawy nowelizującej. Kto z państwa jest za przyjęciem 6. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. W 7. poprawce do art. 4 projektu ustawy nowelizującej wnioskodawcy proponują skreślić pkt 3. Kto z państwa jest za przyjęciem 7. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z państwa jest za przyjęciem 8. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Kto z państwa jest za przyjęciem 9. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Całość. Kto z państwa jest za przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 3113, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich.

Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Czy jeszcze? Nikt więcej się nie zgłasza. Listę posłów zgłoszonych do oświadczeń uważam zatem za zamkniętą. Jako pierwszy ma głos pan poseł Robert Majka, poseł niezależny. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie!

Żadna zasada konstytucji nie zasługuje bardziej na poszanowanie niż zasada wolności myśli. Nie chodzi tu o zapewnienie jej tym, którzy się z nami zgadzają, lecz o to, by mogły z niej korzystać osoby, których poglądów nie znosimy. Dziś, przy końcu roku 2018, prawie po 30 latach ze zdumieniem muszę powiedzieć, że w Polsce nie jest przestrzegany ani art. 54 konstytucji z 1997 r. o wolności słowa ani art. 10 Prawa prasowego, na co posiadam dowody. I nie jest to tylko i wyłącznie zasługa rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Czesława Kiszczaka: My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych.

Mianowicie ostatnio pan prezydent Andrzej Duda, którego nie ma tutaj podczas obrad, uznał, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego pani Gersdorf złamała prawo i że Sąd Najwyższy nie przestrzega prawa, łamiąc również konstytucję. Ale jestem zupełnie zdumiony, że ten sam prezydent Rzeczypospolitej nie składa zawiadomienia do prokuratury, do pana ministra Ziobry, o tym, że sama pani prezes Gersdorf złamała prawo. Dlaczego? Ktoś zapyta, skąd ja to wiem. Odpowiem w ten sposób: otrzymałem pismo od pana prezydenta Dudy, że pani prof. Gersdorf nie jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego.

Środki masowego przekazu zupełnie nie są tym zainteresowane. Ba, złożyłem interpelację do władz Rzeczypospolitej, do pana premiera Mateusza Morawieckiego, i tak jak na wstępie powiedziałem, środki masowego przekazu zupełnie tego nie widzą. Uznają, że tego tematu nie ma. Potwierdził mi to pan prezes Surmacz. Niestety, ale Polska Agencja Prasowa zupełnie nie uznała tego za stosowne, aby przekazać informacje Polakom. To jak Polacy, proszę państwa, Wysoka Izbo, mogą się dowiedzieć prawdy, jeśli po prostu pan prezes Surmacz blokuje informacje Polskiej Agencji Prasowej? Złożyłem interpelację w sprawie ustawy 447, to jest bardzo ważna ustawa. Realizacja tej ustawy grozi państwu polskiemu wydatkami w kwocie 300 mld dolarów. Niestety również ta informacja została przemilczana.

Myślę, że polskie władze, pan prezydent, zgodnie z art. 126 ust. 2, powinny się tą sprawą zająć. Kłaniam się. Bardzo dziękuję. Panie i Panowie Posłowie! W niedzielę, 16 grudnia 2018 r., odbyły się w Puławach uroczystości związane z odsłonięciem pomnika upamiętniającego rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Podczas homilii powiedział m.in.: Kościół w Polsce zachęca w roku liturgicznym, który rozpoczął się w pierwszą niedzielę adwentu, do tego, byśmy w mocy Bożego Ducha czuli się posłani do pełnienia zadań w ojczyźnie i Kościele. Mamy tak jak św. Jan Chrzciciel przygotowywać drogi Chrystusowi do ludzkich serc, prostować kręte ścieżki, wypełniać doliny, równać pagórki, nie powiększać podziałów, jakie są, ale je zasypywać, aby wszyscy ludzie ujrzeli zbawienie Boże. Bezpośrednio po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik, który znajduje się przy Grupie Azoty Puławy, gdzie odbyła się druga część obchodów. Składa się z krzyża, ścianki z napisem „Solidarność” oraz orła w koronie. Symbolika krzyża na tym pomniku jest nieprzypadkowa, jako że krzyże towarzyszyły pracownikom puławskich zakładów od dekad.

Krzyż wisiał na bramie prawie 2 tygodnie. Pracownicy składali pod nim kwiaty, palili znicze i modlili się.

W następnych latach krzyż ten był noszony przez członków „Solidarności” podczas uroczystości kościelnych. Wiosną 1990 r., czyli już w całkiem nowych czasach, w ówczesnym zakładzie mechanicznym zakładów wykonano nowy, stalowy krzyż. Ustawiono go na rozjeździe dróg prowadzących do bramy nr 1 i bramy nr 2. Krzyż ten był wyrazem dziękczynienia za zwycięstwo „Solidarności” i jednocześnie pomnikiem historycznego czynu pracowników, pomnikiem ofiar okresu solidarnościowego zrywu z początku lat 80.

Z przemówień zgromadzeni mogli dowiedzieć się o historii strajku, który odbywał się w puławskich zakładach. Wyłoniono wówczas komitet strajkowy, którego przewodniczącym został Zygmunt Woźny. Według oceny Służby Bezpieczeństwa strajkowało ok. 3 tys. osób. Był to najdłuższy strajk zakładowy na Lubelszczyźnie po wprowadzeniu stanu wojennego.

Podczas tej podniosłej uroczystości aktywny uczestnik wydarzeń z 1981 r. Jan Okoń, który był więziony za udział w strajku, przekazał na ręce przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Grupie Azoty Puławy SA Piotra Śliwy krzyż, który towarzyszył strajkującym, a potem był przechowywany w jego domu. W uroczystości odsłonięcia pomnika udział wzięli uczestnicy strajku, duchowni z ks. abp. Stanisławem Budzikiem, parlamentarzyści lubelscy: Gabriela Masłowska, Krzysztof Szulowski, Włodzimierz Karpiński, Jakub Kulesza, senator Stanisław Gogacz, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, władze samorządowe, reprezentanci władz „Solidarności” i mieszkańcy Puław. Z okazji odsłonięcia pomnika upamiętniającego strajk w Zakładach Azotowych w Puławach wszystkim bohaterom „Solidarności” ziemi puławskiej, wielu już nieżyjącym, składam wyrazy najwyższego szacunku i uznania. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania pomnika. Oświadczenie wygłosi pani poseł Bożena Kamińska, klub Platformy Obywatelskiej. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Tę sprawę kieruję do pana premiera rządu i pana ministra sprawiedliwości pana Ziobro. Jarosław Zieliński, wiceminister, zastraszał, szantażował Policję suwalską, rządził się jak właściciel folwarku. Do prywatnych spraw brał policję jak poddanych. Przez okres ponad 2 lat musieli pełnić służbę dzień i noc przy posesji za pieniądze podatnika. Władze Policji w Suwałkach borykały się z obsadzeniem posterunków służbowych, zabezpieczeniem porządku w Suwałkach, a pan Zieliński brał policjantów jak własnych poddanych.

Dziwne, że ponad 2 lata ten proceder istniał, a pan wiceminister Jarosław Zieliński tego nie widział. Pan Kołnierowicz wydał wyrok i osądził, że winna jest posłanka Kamińska. Szydził, znieważał. Uważam, że premier rządu i minister Ziobro wyciągną odpowiednie wnioski. Pragnę również z tego miejsca, mając na względzie, że wszyscy posłowie dzisiaj otrzymali orędzie Ojca Świętego Franciszka na 52. Oprócz cnót w polityce nie brakuje niestety także wad wynikających zarówno z niekompetencji osobistej, jak i z wypaczeń w środowisku politycznym i instytucjach. Jest oczywiste dla wszystkich, że wady życia politycznego odbierają wiarygodność systemom, w obrębie których polityka jest prowadzona, a także autorytetowi, decyzjom i działaniom ludzi, którzy się jej poświęcają. Te wady osłabiające ideał autentycznej demokracji są hańbą życia publicznego i zagrażają pokojowi społecznemu: korupcja w wielu formach bezprawnego przywłaszczenia sobie dóbr publicznych, instrumentalizacja ludzi, odmawianie praw, brak poszanowania reguł wspólnotowych, bezprawne bogacenie się, uzasadnianie władzy siłą lub arbitralnym pretekstem racji stanu, skłonność okopywania się przy władzy, ksenofobia i rasizm, zaniechanie troski o ziemię, nieograniczona eksploatacja zasobów naturalnych ze względu na doraźny zysk, pogarda dla tych, którzy zostali zmuszeni, by udać się na wygnanie. Ja dedykuję te słowa Ojca Franciszka również wszelkim osobom, które sprawują teraz władzę, a w szczególności nadzorują bezpieczeństwo naszego kraju, czyli służbom mundurowym, Policji i innym. Dziękuję bardzo. Teraz oświadczenie wygłosi pan poseł Jacek Wilk, Wolność i Skuteczni. Wysoka Izbo!

Protesty te biorą się z rozpaczliwej sytuacji polskiego rolnictwa, polskich rolników i są takim krzykiem rozpaczy skierowanym do rządzących, aby w końcu zrozumieli, na czym polega prawdziwy problem polskiego rolnictwa. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, mówiłem, że polskie rolnictwo może być jednym z największych atutów Polski na wspólnym rynku, wszakże pod jednym warunkiem, właściwie pod dwoma warunkami.

Sytuacja niestety jest dokładnie odwrotna.

Wszystko, co rolnik musi kupić od czasu właśnie wejścia do Unii Europejskiej, zdrożało o kilkadziesiąt procent, a nawet nierzadko o drugie tyle.

Dopłaty do rolnictwa, do gruntów rolnych są nadal kilka razy, czasem nawet cztery razy niższe niż w innych państwach. W jaki więc sposób polski rolnik może konkurować z rolnictwem, z rolnikami z innych krajów? Co gorsza, polskie rolnictwo jest zadłużone jak nigdy w historii, ponieważ rolnik, żeby kupić cokolwiek, dostać jakąkolwiek dotację na planowany przez siebie zakup, chociażby maszyn, np. ciągnika, musi zaciągnąć kredyt. W związku z tym polscy rolnicy są zadłużeni jak jeszcze nigdy w historii.

Do tego jeszcze polski rolnik nawet nie może dokonać uboju świń we własnym zakresie, a produkcja chociażby wędlin jest zakazana. Wszystko to powoduje, że sytuacja na polskiej wsi jest coraz gorsza.

Prosi, aby ludzie sami przyjeżdżali i np. zbierali sobie jabłka, bo nie jest w stanie ich sprzedać albo po prostu najzwyczajniej w świecie mu tego nie wolno. Po pierwsze, rolnik zarabia tym więcej, im bliżej sprzedaje swoje produkty finalnemu odbiorcy, a po drugie zarobi tym więcej, im bardziej przetworzony produkt sprzedaje.

Po pierwsze, trzeba tak zmienić prawo, aby rolnik bez żadnych ograniczeń, bez żadnych przeszkód mógł swobodnie sprzedawać we własnym zakresie wszystko to, co sam u siebie wyprodukuje, bez żadnych pośredników i bez żadnych ograniczeń.

Oczywiście musimy też robić wszystko, co się da, aby polski rolnik po prostu miał rynki zbytu. Takie są straty. Niestety musimy się na to przygotować. Dziękuję bardzo.